Wysoka Izbo! Na podstawie regulaminu Sejmu zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia do czasu wprowadzenia do porządku posiedzenia Sejmu punktów obejmujących przeprowadzenie pierwszego, drugiego i trzeciego czytania trzech projektów ustaw złożonych przez Koalicję Obywatelską, w tym projektu senackiego. Mamy ustawy, na które czekają ludzie. Zbyt dużo czasu straciliście, panowie. Zróbmy to teraz. Wiedzieliście o wielu rzeczach, byliście bezczynni, nie mówiliście nam prawdy. Teraz trzeba działać naprawdę bardzo szybko. Wiedzieliście - oskarżam was, tak, wiedzieliście - manipulowaliście, wprowadziliście chaos i po prostu jesteście tchórzami. Tysiące ludzi codziennie naraża swoje życie, pracując bez sprzętu ochronnego, nie ma wystarczającej liczby testów, a wy nie zrobiliście nic. Każdy dzień zwłoki oskarża was. Dlatego nie mówcie nieprawdy, nie kłamcie, tylko weźmy się dzisiaj do pracy, bo to są naprawdę ważne czasy. Nie odkładajmy tego w nieskończoność.

Mamy jeszcze jutro posiedzenie Sejmu, w związku z czym jutro to rozpatrzymy. Rozpatrzymy wniosek formalny, panie pośle. Pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska.

Wysoki Sejmie! Zwracam się z prośbą o przerwanie obrad, zwołanie Konwentu Seniorów oraz wprowadzenie do porządku obrad pierwszego i drugiego czytania uchwały w sprawie wyrażenia wdzięczności pracownikom służby zdrowia. Ci ludzie dzień w dzień narażają swoje życie i zdrowie: pracownicy służb medycznych, pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, a także pracownicy socjalni.

Dziękuję, pani poseł. Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni całej służbie zdrowia, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale pani doskonale wie, że jest to wniosek nieregulaminowy.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mniej sporów proceduralnych, więcej działania. Polscy pracownicy, polscy przedsiębiorcy oczekują natychmiastowego przyjęcia pakietu antykryzysowego. Zgłaszamy swoją ustawę, dobrowolny ZUS, zgłosiliśmy pakiet antykryzysowy, propozycję minimalnej pensji dla wszystkich pracowników, nieoprocentowane kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego, szybki zwrot VAT-u, pomoc dla pracowników i dla pracodawców. Zróbmy użytek z tego, że przyjechali tutaj posłowie, ogłośmy przerwę. Jest to na razie tarcza tekturowa, ale może być tytanowa po wprowadzeniu naszych poprawek. Wzywam wszystkich do przyjęcia dzisiaj ustaw związanych z pakietem antykryzysowym. Bez tego nasze spotkania nic nie znaczą dla społeczeństwa.

Wszyscy wiemy, że trzeba to zrobić bardzo szybko. Na to jest przeznaczony jutrzejszy dzień. Państwo doskonale widzieliście, że dzisiaj na skutek braku porozumienia.

Proszę wicemarszałka Sejmu pana Ryszarda Terleckiego o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Prezydium Sejmu zgłaszam projekt zmiany regulaminu Sejmu umożliwiającej posłom zdalne procedowanie nad ustawami. Po wprowadzeniu przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii na całym świecie konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków funkcjonowania parlamentu Rzeczypospolitej, Sejmu Rzeczypospolitej, ale także zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia pracowników Sejmu, jak również uchronienie się przed sytuacją, gdy Sejm zbierze się tu w całości, a następnie posłowie rozjadą się do swoich okręgów. W razie gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa w całym kraju. Wysoki Sejmie!

Zwrócę tylko uwagę, że w tej chwili w całej Europie parlamenty przyjmują nadzwyczajne środki ostrożności, w tym także Parlament Europejski, i zmieniają swoje regulaminy. Panie pośle, bardzo proszę o nieprzeszkadzanie.

Wnoszę o to, aby Wysoka Izba przyjęła ten regulamin dzisiaj, tak abyśmy mogli zdalnie procedować w ciągu następnych dni. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Jako pierwszego proszę pana posła Krzysztofa Sobolewskiego, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mam zaszczyt w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić stanowisko w związku z przedmiotową uchwałą. Projekt zmiany regulaminu Sejmu, zawarty w druku nr 286, zaproponowany w pełnym konsensusie przez Prezydium Sejmu, dotyczy zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana ta miała na celu i ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Pan marszałek sprawozdawca przedstawił zakres zmian, jakie owa uchwała miałaby objąć. W związku z obecną sytuacją epidemiczną konieczne jest wprowadzenie zmian w regulaminie Sejmu, które regulowałyby te sprawy. Mógłbym długo uzasadniać konieczność podjęcia takich, a nie innych kroków i zmian w regulaminie Sejmu, ale nie jest to czas na takie wystąpienia. Dla Prawa i Sprawiedliwości zdrowie i życie Polaków jest ważniejsze niż sztywne normy prawa.

Prawo, które nie służy narodowi, to bezprawie. Panie Premierze! Zmiany, które są proponowane, a są zawarte w tym druku, dostosowują regulamin Sejmu do bezprecedensowej sytuacji, w której znalazła się Polska, a która to sytuacja nie miała wcześniej miejsca we współczesnej historii naszej ojczyzny. Dziękuję, panie pośle. Teraz proszę pana posła Borysława Budkę, Koalicja Obywatelska.

Szanowni Państwo! Przyjechaliśmy tutaj dla was, bo wy nas wybraliście. To jest wydłużenie świadczeń na ubezpieczenia społeczne dla was, którzy dzisiaj opiekujecie się swoimi dziećmi, bowiem zamknięte są szkoły, przedszkola i żłobki. To są projekty, które zapewniają bezpieczeństwo milionom osób. To jest m.in. minimalne wynagrodzenie dla każdego, kto dziś nie może pracować. Nie dzielimy ludzi na lepszy i gorszy sort. Chcemy pomagać wszystkim, bo taka jest rola państwa. Żaden Polak, żadna Polka, żaden przedsiębiorca, żaden pracodawca nie powinni być dotknięci skutkami tego kryzysu. A my, parlamentarzyści, jesteśmy od tego, by przyjąć właśnie takie regulacje. Zaproponowaliśmy 20 mld zł na służbę zdrowia. To są konkretne pieniądze na środki ochrony osobistej dla was, drodzy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy dzisiaj w skrajnych warunkach bronicie naszego życia, a niestety ten rząd nie potrafi wyposażyć was nawet w podstawowe środki ochronne. To są konkretne środki na to, by zakupić sprzęt dla szpitali. To są również konkretne środki na to, by każdy, kto miał kontakt z koronawirusem, mógł być bardzo szybko przebadany, byśmy przyjęli dobre wzorce krajów, które skuteczniej aniżeli Włochy radzą sobie z koronawirusem. Tymczasem co proponuje obecna większość? Obecna większość chce, byśmy dzisiaj zajmowali się tylko i wyłącznie komfortem pracy parlamentarzystów. My zostaliśmy wybrani na trudne czasy. My jesteśmy po to, by służyć wam. Przyjechaliśmy dlatego, że miliony z was dzisiaj poszły do pracy, że dzisiaj każdy, kto jest w pracy, oczekuje pomocy od państwa, pomocy od nas, parlamentarzystów. My nie uchylamy się od pracy, bo my zostaliśmy wybrani przez was i dla was. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi. To dziś zwalniani są polscy pracownicy. To dziś upadłość ogłaszają kolejni przedsiębiorcy, kolejni pracodawcy. Nie chcemy wojen regulaminowych. Chcemy pracować dla was. Zjawiliśmy się w Sejmie, bo nie tchórzymy, bo jesteśmy po to, by w momentach krytycznych pracować dla was. Będziemy robić wszystko, by to, co wyjdzie z tego Sejmu, było w poczuciu odpowiedzialności za wasze bezpieczeństwo. Proszę bardzo, głos ma pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zebraliśmy się jako parlamentarzyści w godzinie próby. Zebraliśmy się w poczuciu odpowiedzialności za państwo, konstytucję, każdą Polkę i każdego Polaka. Lewica była, jest i zawsze będzie do dyspozycji obywateli. Złożyliśmy projekty ustaw i przedstawiliśmy pomysły, jak dzisiejszą sytuację uzdrowić, co zrobić, żeby miliony polskich przedsiębiorców czuło, że nie zostali pozostawieni sami sobie. Jesteśmy tutaj, bo pracownicy w całej Polsce zdają sobie sprawę, że już za kilka dni mogą nie dostać wynagrodzeń, a na koniec kwietnia będą miliony pozostawione bez złotówki na kontach. Lewica mówi o swoich propozycjach jasno i wyraźnie. Mają być zatrzymane raty kredytów: nie na 3 miesiące, ale na minimum 6 albo 9 miesięcy. Mamy doprowadzić do sytuacji, w której ZUS zostanie wstrzymany i nikt nie będzie musiał za niego dopłacać. Chcemy, żeby przedsiębiorcy byli zwolnieni z ZUS-u. Chcemy, żeby państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za rachunki za gaz, prąd, najem. Chcemy o to walczyć i w poczuciu odpowiedzialności dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. To również odpowiedzialność za pracowniczki i pracowników tego gmachu, za te tysiąc osób, które dzisiaj tutaj z nami są. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Będziemy walczyli o każdą złotówkę, będziemy walczyli o każdy grosz, żebyście byli doposażeni, żeby w polskich szpitalach nie brakowało maseczek i testów, żeby polska służba zdrowia pamiętała o tym, kto w godzinie próby był razem z wami. Ale odpowiedzialność to również myślenie o Polsce, która potrzebuje zmiany. Polscy parlamentarzyści muszą pracować, ale muszą też mieć do tego możliwości. Odpowiedzialność nakazuje zmienić regulamin Sejmu tak, żebyśmy mogli to prawo, które chcemy zmieniać, bo wierzę, że cała opozycja i cała koalicja chce to robić, mogli zmieniać. Dzisiaj nie ma zgody na to, żebyśmy kryzys wykorzystywali do politycznych kłótni. Dzisiaj nie ma koalicji i opozycji. Dzisiaj nie ma rządu, polityczek i polityków. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Polakami odpowiedzialnymi w imię konstytucji i naszych mandatów za to, żeby Polska była Polską, żebyśmy ją uratowali z tego kryzysu. Lewica tego słowa dotrzyma.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W czasach próby, w czasach kryzysu, w czasach epidemii dwie postawy są kluczowe: postawa solidarności i odpowiedzialności. To jest test dla każdego z nas, dla każdego z nas, Polaków, czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, za najbliższych. Instytucje państwa zawiodły. Nie przygotowaliście państwa na czas epidemii, na czas kryzysu. Jeszcze nie tak dawno główny inspektor sanitarny mówił: wirus jest w Chinach, a Chiny są przecież bardzo daleko. Nie przygotowaliście służby zdrowia, nie przygotowaliście schematów postępowania i działań. To jest gigantyczne zaniedbanie.

Instytucje państwowe do tej pory nie zdawały egzaminu, bo nas nie przygotowały do kryzysu, ale zdali egzamin Polacy, bo zachowują się, po pierwsze, odpowiedzialnie, zdali egzamin pracownicy ochrony zdrowia, pielęgniarki, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, zdają egzamin pracownicy ochrony zdrowia i funkcjonariusze służb mundurowych. Musimy dzisiaj ich wesprzeć, żeby miejsca pracy nie zostały utracone. Tu jest też potrzebna solidarność i zrozumienie, bo jak słyszę ze strony Platformy, że chce zakończenia wojenek, a sama za każdym razem szuka okazji. do sporu politycznego i upolitycznienia tego. To nie jest dobra droga. Dla was święte są regulaminy, a nie sprawy pracowników i przedsiębiorców. Tak, zdrowie i życie na pierwszym miejscu, pracownicy i przedsiębiorcy, dokładnie tak. Trzeba przyjąć dobrowolny ZUS, trzeba dać nieoprocentowane kredyty, minimalną pensje dla pracowników, którzy może są już na urlopie bezpłatnym, może są już zwalniani. Zdajmy sobie wszyscy sprawę, że 2 mln Polaków może stracić pracę. Zdajmy sobie sprawę, że 70% firm może zwalniać pracowników, że mogą upadać z dnia na dzień od najmniejszej do największej. To jest nasza odpowiedzialność. Miarą odpowiedzialności i solidarności jest też umiejętność dzisiaj rozmowy i współpracy, stawiania warunków, bo bezkrytyczne przyjmowanie tego, co proponuje rząd, to jest tylko i wyłącznie skazanie nas na tekturową tarczę, a ona musi być tytanowa i musi być jak najszybciej przyjęta.

Panie pośle Grupiński, pan sobie pozwala na uwagi kompletnie niestosowne. Jesteście państwo jedynymi posłami na tej sali, którzy pohukują, którzy przeszkadzają. Jeszcze raz apeluje, panie pośle. Proszę nie dyskutować ze mną. Każdy ma prawo zabrać głos. Proszę nie przeszkadzać. Jeśli będzie pan chciał zadać pytanie, będzie pan miał szansę. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Premierze! Członkowie Rządu! Panowie Prezesi! Przewodniczący Klubów i Partii Politycznych! Jesteśmy w sytuacji szczególnej, która wymaga od nas powagi, a nie przekrzykiwania się tutaj w Izbie. Jesteśmy w sytuacji, w której nasze państwo i klasa polityczna reprezentująca nasze społeczeństwo toczą wojnę na trzech frontach. Pierwszy front to oczywiście walka z epidemią o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Drugi front, do którego rząd przygotowuje się, dziś w nocy skończył prace nad ustawami, a dziś rano mieliśmy uczestniczyć w konsultacjach, które zostały przełożone na popołudnie i wieczór, to walka z kryzysem o źródła utrzymania dla polskich obywateli i przetrwanie polskich przedsiębiorstw. Trzeci front, który nas tutaj zgromadził, to walka ze słabością naszego państwa, które okazuje się nieskuteczne i które potyka się o własne nogi, chcąc walczyć w takiej kryzysowej sytuacji. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak to się stało, że musimy spotkać się tutaj, żeby nowelizować w kryzysowej, epidemicznej sytuacji regulamin Sejmu. Otóż nikt nie przewidział takiej okoliczności, nikt nie przygotował systemu technologicznego do obrad on-line. Dzisiaj znowelizujemy regulamin, jutro zderzymy się z ograniczeniami systemów, które albo ze sobą nie współpracują, albo nie istnieją. Jak to się stało? Siedzi tutaj pomiędzy nami marszałek Kuchciński, który był marszałkiem Sejmu w latach 2017–2018, kiedy był przeprowadzony przetarg na nowy system liczenia głosów, przetarg, który po roku prób został zdemontowany, bo ten system nie działał. Ale siedzą tutaj również były marszałek Schetyna, była pani marszałek Kidawa-Błońska, którzy również, kiedy pełnili ten urząd, nie wdrożyli tu nowoczesnych systemów, nie zaproponowali nowelizacji regulaminu Sejmu, którą dzisiaj uchwalimy. Nasza postawa jest konstruktywna, bo jesteśmy opozycją merytoryczną. Przedstawimy poprawki do regulaminu Sejmu, poprawki, w myśl których chcemy te nadzwyczajne przepisy powiązać ze stanem nadzwyczajnym. Uważamy, że zawieszenie normalnego obradowania Sejmu jest uzasadnione w sytuacji stanu nadzwyczajnego. Tak mówią konstytucjonaliści, również się z tym zgadzamy. Chcemy pracy merytorycznej, skutecznej, efektywnej, nowoczesnej. Chcemy takiej pracy. Chcemy, żebyśmy mogli normalnie, legalnie obradować, uchwalać prawo, na które czekają obywatele. Bardzo apelujemy: uwzględnijcie wszyscy państwo te poprawki, które przedstawiamy, poprawki do regulaminu Sejmu, i przejdźmy natychmiast do dyskusji o tarczy antykryzysowej, przejdźmy do dyskusji o ustawach, które dziś w nocy skończył pisać rząd. Nie skupiajmy się tutaj na przekrzykiwaniu się, kto lepiej czy gorzej coś powiedział, bo to obywateli kompletnie nie interesuje. Ostatnia sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę. Szanowni państwo, nie możemy mówić obywatelom, że mają pozostać w domu, a jednocześnie zmuszać komitetów wyborczych, żeby wydelegowały dziesiątki tysięcy ludzi do komisji na szkolenia i żebyśmy uczestniczyli w organizacji wyborów. Panie premierze, panie prezydencie - jeśli prezydent lub jego personel nas ogląda - przesuńmy wybory. Bardzo o to apeluję. Nie zmuszajmy nas do tego, żebyśmy w tej chwili dalej pracowali nad wyborami. Informuję panie i panów posłów, iż Prezydium Sejmu na podstawie art. 39 ust. 1 regulaminu Sejmu ustaliło w tym punkcie limit pytań: po jednym dla każdego z klubów i koła oraz posła niezrzeszonego. Do pytania zgłosiła się tylko jedna osoba, pan poseł Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie dlatego że jest niebezpiecznie, tylko dlatego że wy nie chcecie odpowiadać na pytania, nie chcecie słuchać trudnych pytań i nie chcecie ludziom udzielić informacji, nie chcecie odpowiedzieć. Wy mówicie, że ilość maseczek, którymi dysponujecie w Polsce, to jest tajna informacja. Testów nie ma, maseczek nie ma. Zamiast uspokoić ludzi, że je macie, to mówicie, że to jest tajna informacja. Nie macie tego sprzętu, a my mamy obowiązek mówić. Czy pan premier tu dzisiaj zabierze głos i powie, kiedy odda VAT, który jest przedsiębiorców, a po prostu im go wolno oddajecie? Czy pan premier powie, dlaczego kazaliście ludziom płacić w tym miesiącu ZUS? Przecież mogliście powiedzieć: Wstrzymajcie się z tym ZUS-em, nie płaćcie, zapłaćcie swoim pracownikom.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Padły tutaj bardzo dziwne słowa pani marszałek Kidawy-Błońskiej, paru osób, które zabierały głos - że kłamiemy, że zatajamy informacje o liczbie testów. Albo państwo nie słuchacie mediów, albo państwo nie chcecie ich słuchać, albo państwo wprowadzacie w błąd wszystkich Polaków. O liczbie testów, które rozdysponowaliśmy do wszystkich laboratoriów, mówię od wielu, wielu dni: 100 tys., 200 tys., 500 tys., maseczki, testy, rękawiczki. Oczywiście można tego nie słuchać, można mówić, że wprowadzamy Polaków w błąd. Myślę, że Polacy nas ocenią w tym zakresie. Jeżeli mówimy o tym, ile testów rozdysponowaliśmy po laboratoriach, mówimy o tym regularnie: 100 tys. testów już poszło do laboratoriów, kolejne 50 paskowych będzie wprowadzone jutro. Naprawdę tutaj nic nie próbujemy zatajać, nic nie próbujemy oszukiwać. Wydaje mi się, że takie uwagi w sytuacji dzisiejszej, w jakiej jest Polska, są po prostu trochę nie na miejscu. Natomiast, szanowni państwo, wydaje mi się, że sytuacja dzisiejsza, kiedy wszyscy się gromadzimy na tej sali. Patrzę na tę salę parlamentu, gdzie siedzimy w odległości kilku metrów od siebie. Szkoda, że nie doszliśmy do konsensusu, że możemy to zrobić zdalnie. Część z państwa nosi maseczki, rękawiczki. Oczywiście każdy ma prawo bać się o siebie, każdy ma prawo odczuwać strach, bo sytuacja jest niecodzienna. I myślę, że to jest czas, kiedy zamiast dyskutować partyjnie, dyskutować politycznie, co kto komu zarzuca, powinniśmy raczej dyskutować, w jaki sposób tak usprawnić nasz system, tak kierować tym systemem, gospodarczym, publicznej służby zdrowia, prywatnej służby zdrowia, wszystkich medyków, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby wprowadzać atmosferę taką. Bo nie będzie świetnie, będzie wzrastała liczba chorych, będziemy mieli coraz więcej osób umierających. Tak jest wszędzie. Jedyne, co my możemy zrobić, to ograniczyć tę liczbę, ograniczyć poprzez nieprzychodzenie w miejsca, gdzie nie musimy przychodzić, niechodzenie po ulicach, chodzenie do pracy, gdzie jest to niezbędne. Są miejsca, gdzie musimy pracować. Natomiast, szanowni państwo, myślę, że czas jest na to, żebyśmy wszyscy wspólnie starali się wypracować najlepsze mechanizmy, które obronią polską gospodarkę, które obronią nas wszystkich, w tym ochronią i naszą służbę zdrowia. Żadne instytucje, w tym instytucje międzynarodowe, nie zapewniły nam na dzisiaj środków ochrony osobistej.

I bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, bo tacy są, którzy pomagają nam, pomagają nam wszystkim, pomagają szpitalom, pomagają medykom, pomagają laboratoriom, ale też w transporcie miejskim, pomagają w kateringu dla miejsc, które muszą pracować, żebyśmy wszyscy wyszli z tego obronną ręką. Za to bardzo dziękuję. Myślę, że czas jest na to, żeby szybko przeprocedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo, i myślę, że dzięki temu, dzięki bardzo racjonalnej i odpowiedzialnej postawie, będziemy mogli funkcjonować jako Polska, jako polski naród w kolejnych latach. Dziękuję, panie ministrze.

W imieniu klubu Konfederacji chciałbym zadać pytanie o to, jak wygląda stan przygotowania technicznego Kancelarii Sejmu do organizacji obrad on-line. Jeżeli mamy przyjąć taki schemat i taki scenariusz i omówić tarczę antykryzysową jutro w formule on-line, to wypada, żebyśmy otrzymali informację, czy jest gotowość techniczna. Pytanie co do nowelizacji regulaminu, szczegółowe, związane z naszymi poprawkami: Dlaczego regulamin Sejmu wyklucza w formule on-line udział ekspertów, czynnika społecznego w obradach komisji, kiedy formuła on-line właśnie to ułatwia i pozwala łączyć się z ekspertami w dowolnym miejscu w dowolnym czasie? Przy władzy pani marszałek nad tym, jak będą przebiegać obrady, nie ma właściwie żadnego problemu, żeby ten czynnik społeczny uwzględniać, a właśnie przy dyskusji nad tarczą szczególnie ten głos środowisk gospodarczych, środowisk społecznych mógłby być dla nas istotny. Tak że pytanie jest takie: Dlaczego próbujemy wykluczyć w tej nowelizacji regulaminu czynnik społeczny? Czy może warto uwzględnić poprawkę Konfederacji, żeby ten czynnik społeczny przywrócić? Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do drugiego czytania. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? Zgłosili się posłowie. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! My dzisiaj nie powinniśmy zajmować się regulaminem Sejmu. Dzisiaj powinniśmy już w tej chwili pracować nad rozwiązaniami, które będą ratunkiem dla polskiej służby zdrowia, ale również dla was, którzy boicie się o swoje miejsca pracy, boicie się o swoich najbliższych.

My byliśmy gotowi do pracy. Uważamy, że formuła, która została zaproponowana, była niedopuszczalna z uwagi na to, że po prostu takich rozwiązań pani marszałek wcześniej nie przygotowała. Składamy poprawki do regulaminu Sejmu, wierząc w to, o czym mówią dziś rządzący: że to ma być rozwiązanie czasowe. Ale chcę was zapewnić, że bez względu na to, w jaki sposób większość rządząca będzie prowadzić obrady, nie zapomnimy o was. Będziemy zgłaszać te wszystkie postulaty, o których mówicie. Nie może być tak, że polscy pracownicy będą dzieleni na lepszych i gorszych, nie może być tak, że pracodawca, który ma więcej niż dziewięciu pracowników, będzie miał inną pomoc aniżeli ten, który zatrudnia do dziewięciu. Wreszcie nie może być tak, że minister zdrowia dzisiaj tutaj wychodzi i nie chce rozmawiać o 20 mld zł. My jesteśmy dla pana, my chcieliśmy pomóc, my chcieliśmy właśnie pomóc polskiej służbie zdrowia, my chcieliśmy przeznaczyć pieniądze tu i teraz, żeby pan mógł lepiej działać, żeby nie musiał pan każdego dnia wymieniać innych liczb, jeśli chodzi o sprzęt, by nie musiał pan gasić pożarów, które są codziennie w polskich szpitalach.

Nie było pańskiej zgody na to, żeby w takim trybie obradować, i nie było zgody Konfederacji, dlatego spotykamy się dzisiaj, żeby zmienić regulamin właśnie na skutek pańskiego stanowiska. Nie było konsensusu i nad tym ubolewam, bo gdyby ten konsensus był, dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym punkcie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią poseł Annę Marię Żukowską, klub parlamentarny Lewica. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Lewica poważnie podchodzi do kryzysu, jaki w tej chwili mamy w kraju, i uważamy, że parlament musi mieć możliwość kontroli w stosunku do rządu i dlatego chcemy zachowania możliwości funkcjonowania parlamentu również w takiej sytuacji, kiedy niestety niektórzy z nas być może zostaną zarażeni i będą musieli odbywać kwarantannę. Dlatego uważamy, że projekt dotyczący możliwości zdalnego głosowania, zdalnego odbywania posiedzeń izby niższej parlamentu jest projektem absolutnie koniecznym.

Nie mamy pełnego zaufania do Prawa i Sprawiedliwości i uważamy, że w takiej sytuacji, kiedy głosowanie i posiedzenie odbędą się w formie zdalnej, musimy mieć możliwość większego konsensusu. Chcemy zmienić brzmienie tak, żeby to Prezydium Sejmu kwalifikowaną większością głosów, a nie marszałek Sejmu, decydowało o przeprowadzeniu posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość - po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Taka jest nasza propozycja, jedna z tych, które będę zgłaszała.

Mówimy tutaj o systemie teleinformatycznym, w jakim będziemy się poruszali i w jakim będziemy procedowali na tych posiedzeniach. Nasze poprawki mają na celu zachowanie bezpieczeństwa obrad i - tak jak mówię - uniemożliwienie stworzenia jakichś nowych projektów, które wcześniej nie były uzgodnione na posiedzeniu Prezydium Sejmu. Dziękuję, pani poseł, dziękuję, tylko, pani poseł, chciałam powiedzieć, że to nie był regulamin przedstawiony przez klub Prawo i Sprawiedliwość, tylko wszystkie kluby znały ten regulamin dużo wcześniej, przyjęliśmy go jednomyślnie, więc był czas na to, żeby naprawdę.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W imieniu Koalicji Polskiej kilka spraw.

Te poprawki składamy i prosimy o ich przyjęcie. Najważniejsze jest to, co przyjmiemy w tarczy antykryzysowej. Stawiamy swoje warunki, przesłaliśmy je do kancelarii pana premiera. Po pierwsze, umorzenie podatków i składek, nie tylko dla małych przedsiębiorstw, ale dla tych, które są dotknięte kryzysem. Po drugie, jak najszybszy zwrot VAT-u, bo firmy czekają na te pieniądze. Szybkie linie kredytowe. Pomoc samorządom - to jest kwestia kluczowa. Samorządy sobie nie poradzą bez wsparcia państwa, bo chcą umorzyć podatki od nieruchomości, ale muszą mieć rekompensaty. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wprowadzili też pakiet zdrowotny, pakiet rozwiązań dla służby, dla ochrony zdrowia.

To są gigantyczne problemy pacjentów, którzy nie wiedzą, jak się mają poruszać w tej sytuacji. Tu mam prośbę do pana ministra, korzystając z tej okazji, żeby był pożytek z tego spotkania, żeby poinformował choćby kobiety ciężarne, pacjentów onkologicznych, jak mają postępować i gdzie mają się zgłosić. Kwestie rolnictwa, na początku nieporuszane, po naszych interwencjach są wreszcie w projekcie, ale muszą być jeszcze bardziej rozwinięte. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Proszę, pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Pani Marszałek! W pierwszej kolejności zgłaszam formalnie trzy poprawki przygotowane przez prawników Konfederacji do nowego regulaminu Sejmu. To jest ograniczenie stosowania obrad zdalnych, obrad on-line wyłącznie do trwania stanów nadzwyczajnych. Łączymy to z apelem o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, o nierobienie tego na raty, co samo w sobie może być deliktem konstytucyjnym, jeżeli celowo używa się instrumentów nadzwyczajnych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego łączącego się automatycznie z odsunięciem wyborów o 3 miesiące. Trzecia poprawka dotyczy dopuszczenia czynnika społecznego do obrad on-line. Chciałbym krótko uzasadnić szczególnie tę trzecią sprawę. Jest rzeczą symptomatyczną, że tak długo przygotowywany przez rząd pakiet antykryzysowy był dziś w pierwszej kolejności konsultowany nie ze środowiskami gospodarczymi, ze środowiskami przedsiębiorców, ale z dziennikarzami. Ta zaplanowana dziś rano i odwołana konferencja z przedstawicielami opozycji została zastąpiona przez spotkanie szefa funduszu rozwoju, pani minister i pani prezes ZUS z dziennikarzami. To charakterystyczne, dlatego że cała historia tarczy antykryzysowej rozpoczęła się od zamieszczenia ogłoszeń w prasie z informacją o wirtualnej kwocie 200 mld. Przedsiębiorcy czekają na skonsultowanie z nimi tych propozycji. Cieszymy się, że postulat Konfederacji z poprzedniego roku dobrowolnego ZUS-u został częściowo przyjęty przez rząd, częściowo przyjęty przez partie opozycyjne. To wielki postęp, ale w zbyt małym stopniu. Instrumenty takie jak dopłaty do pensji po 3 czy 4 miesiącach, bo tak to realnie zadziała. Jeżeli mamy 2 miesiące straty obrotu, w trzecim miesiącu będzie rozpatrywanie wniosku, to kiedy to przyjdzie do przedsiębiorstw? Kopiowanie systemu grantów unijnych w przypadku walki z kryzysem to całkowicie błędna ścieżka. To próbują, panie premierze, powiedzieć wam przedsiębiorcy. Konfederacja wyraża ich głos.

Kto jeszcze? Pani Barbara Nowacka i pani Daria Gosek-Popiołek, tak? To oprócz tych dwóch osób pan poseł Nitras, tak?

Myślę, panie pośle, że doskonale zrozumiałam. Proszę bardzo. Pani Marszałek! Otóż niestety, ale z ubolewaniem stwierdzam, że kolejny raz wprowadza pani opinię publiczną w błąd. Zaproponowaliście na posiedzeniu Prezydium Sejmu coś absolutnie niezgodnego z regulaminem, z konstytucją. Prosiliśmy was, błagaliśmy was: zajmijmy się konkretnymi projektami ustaw. Nasz sprzeciw na posiedzeniu Prezydium był tylko i wyłącznie dlatego, że obawiamy się, że przyjęte w sposób niezgodny z prawem prawo będzie później przez was kwestionowane, że ZUS odbierze te zasiłki, które dzisiaj zostaną dane, że gdy zabraknie wam pieniędzy w tym wydmuszkowym budżecie, sięgniecie po raz kolejny do kieszeni polskich podatników. Nie ma zgody na to, żeby prawo było uchwalane w sposób urągający jakimkolwiek zasadom. Pokazaliśmy dzięki naszemu sprzeciwowi, że da się pracować. Jesteśmy dzisiaj w różnych salach, gotowi do pracy dla Polaków. Nie trzeba było tego sprostowania. Przystępujemy do pytań. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! My naprawdę chcemy pracować. Chcemy pracować merytorycznie i chcemy pracować nad ustawami. Ale, pani marszałek, przecież to jest nieprzygotowane. Wysłaliście nam wczoraj w jednym mailu otwartym tekstem hasło i login. Każdy może się włamać, każdy może się włamać na serwer. Ułożyliście hasła, które zdekoduje 17-letnie dziecko bez problemu. Pani marszałek, czy w taki sposób zapewnicie bezpieczeństwo naszego głosowania? Nie traktujemy się poważnie. Mówi rząd: mieliśmy tyle czasu, przygotowaliśmy wszystko, od wielu miesięcy pracujemy. W szpitalach nie ma kombinezonów, przedsiębiorcy nie mają zapewnionych pieniędzy, ludzie tracą pracę, brakuje maseczek, brakuje testów i okazuje się, że system do głosowania zdalnego jest zwyczajnie dziurawy i niebezpieczny.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! To posiedzenie jest wyjątkowe i pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli Sejmowi pracować zdalnie. To ważne, jeśli nie chcemy blokady całego państwa, jeśli chcemy zachować tę ważną funkcję parlamentu, jaką jest patrzenie na ręce rządowi. A więc pytam: Dlaczego państwo nie chcecie się zgodzić, by marszałek zwoływał takie posiedzenia, posiedzenia zdalne, jedynie za zgodą Konwentu? Proponujecie, by marszałek Sejmu jedynie zasięgał opinii. To fatalne rozwiązanie, niedemokratyczne, które prowadzić może do szeregu niedemokratycznych działań i nieprawidłowości. Dlatego szanujmy demokrację, szanujmy polski parlamentaryzm, szanujmy obywateli i obywatelki i zmieńmy ten zapis. I drugie pytanie: Jaki jest stan przygotowania systemu do jutrzejszych obrad zdalnych i jak wygląda zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego tego posiedzenia? Wiemy, że są z tym trudności, dlatego chcemy wiedzieć, jak to (Dzwonek) w tym momencie się kształtuje. Dziękuję, pani poseł. My jesteśmy jako parlamentarzyści zasypywani codziennie informacjami od ludzi, prośbami od obywateli. Naszym obowiązkiem jest przekazywać to wam jako rządzącym. Nasze relacje polegają na tym, że wychodzi pan premier w telewizorze, opowiada i nie odpowiada na pytania. My nie możemy wam zadać pytania. Nie, parlamentarzyści wszystkich klubów siedzą w tym budynku, a wy posadziliście parlamentarzystów PiS-u w zupełnie innym budynku. Padają wnioski o to, żeby sprawdzić kworum, bo my nie wiemy, ilu nas jest. Pani marszałek udaje, że tego wniosku nie ma, nie słyszy tego wniosku. My się boimy manipulacji. My nie wiemy, czy wy nie nadużyjecie prawa, które sobie sami w tej chwili, nie wiadomo czy zgodnie z prawem, przyznajecie. Pan nawet nie próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli ten regulamin przejdzie, my boimy się tego, że wy nie będziecie Polakom. Zapewniam, że kworum mamy. Po przerwie, po zliczeniu podam państwu. Za chwileczkę powiem. W związku z tym, proszę państwa. Tak, jeszcze chwileczkę. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu uchwały poprawki, proponuję, aby Sejm przystąpił do głosowania po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia zgłoszonych poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Zarządzam przerwę w obradach do godz. 15.40.

Wznawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 1. porządku dziennego. Ale już teraz bardzo proszę. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu uchwały. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone. Przystępujemy do trzeciego czytania. Posłów sekretarzy proszę o doliczenie swojego głosu do głosów oddanych w wyznaczonej sali. Proszę panie i panów posłów o trzymanie w trakcie głosowania podniesionych rąk przez czas umożliwiający obliczenie głosów. Proszę bardzo, wniosek formalny. Otóż w związku z tym, że głosujemy w tak szczególnym trybie, proszę o to, żebyśmy wszyscy dowiedzieli się, ilu jest posłów w salach w Sejmie.

To jest kluczowe, żebyśmy wiedzieli, czy Sejm jest w stanie w ogóle podejmować tę decyzję.

Czy Agencja Wywiadu rzeczywiście uprzedzała rząd, że zagrożenie pandemią jest tak poważne? Podobno te ostrzeżenia były w styczniu kierowane do rządu i zostały zlekceważone. Myślę, że warto, żeby pan premier czy któryś z ministrów w tym czasie odpowiedział, ale teraz proszę panią marszałek o podanie liczby posłów w poszczególnych salach w Sejmie. Jest kworum. Panie pośle, przypomnę, że jak mamy normalne posiedzenie Sejmu, to nie wchodzi pan na mównicę i nie pyta, ilu posłów podpisało listę obecności. Dziękuję bardzo. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi, choćby najkrótszej, ale konkretnej, o stopień przygotowania Kancelarii Sejmu do prowadzenia od jutra obrad on-line. Jeżeli dzisiaj mamy to przegłosować, to musimy wiedzieć, bo od tej decyzji bardzo wiele zależy - albo paraliż procesu uchwalania tarczy antykryzysowej, albo sprawne przeprowadzenie jutro obrad w tej sprawie. Tak że prosiłbym o niepomijanie milczeniem pytań w tej sprawie i udzielenie nam informacji, czy to przez odpowiednich pracowników Kancelarii Sejmu, czy przez samą panią marszałek, jeżeli jest w tej sprawie poinformowana. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Obradujemy w szczególny sposób. W szczególny sposób również mamy przedstawić państwu wyniki tego głosowania. Pani marszałek, otrzymałem formularze, które jako poseł sekretarz, lecz również jako jednoosobowa komisja skrutacyjna mam wypełnić, ale prosiłbym panią marszałek o dostarczenie mi listy obecności ze wszystkich sal, tak abym mógł stwierdzić - i przekazać pani marszałek do odczytania wyniki głosowania - że faktycznie taka liczba osób jest obecna w tych salach i bierze udział w głosowaniu.

Jest to niezbędne, abyśmy mogli - także jako ci, którzy biorą udział w głosowaniu - wiedzieć, że nasi koledzy parlamentarzyści również faktycznie w tych salach głosują. Jeśli pani marszałek będzie uważała za stosowne, jestem również do dyspozycji, aby przejść i z innymi sekretarzami stwierdzić obecność tych posłów na sali. Panie pośle sekretarzu, otrzyma pan oczywiście protokoły z każdej sali i możemy przełączyć telebim na salę, w której się odbywają głosowania, jeżeli to będzie potrzebne. Jeżeli pan chce listę obecności, możemy też listę obecności dostarczyć. Oczywiście za chwileczkę udzielę wszystkich informacji dotyczących tego systemu i jutrzejszego posiedzenia, po przegłosowaniu tych poprawek, żebyście wszyscy państwo wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Tylko na początek chciałam na jedno zwrócić uwagę, panie pośle. Jeżeli państwo przeczytaliście ten regulamin - w regulaminie jest wyraźnie powiedziane, że posłowie, którzy chcą uczestniczyć w obradach tu, w parlamencie, mają do tego prawo. Jeśli będą chcieli z tego skorzystać, będą rozmieszczeni tak jak dziś w innych salach, a ci, którzy nie mogą z różnych powodów brać udziału w posiedzeniu parlamentu, będą mogli to robić zdalnie. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 2. i 3. Przystępujemy do głosowania.

Troszkę dłużej to potrwa, bo w tamtych salach jest więcej osób, więc chwileczkę będzie to trwało, w wolniejszym tempie.

Kto z państwa jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę posłów sekretarzy o obliczenie wyników głosowania.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał? Proszę posłów sekretarzy o obliczenie wyników głosowania i przekazanie protokołu

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę.

jest przeciw? Kto się wstrzymał?

371 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę.

jest przeciw?

Kto się wstrzymał? Proszę posłów sekretarzy o obliczenie wyników głosowania i przekazanie protokołu

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 6. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę.

367 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Pani Marszałek! To jest oczywista pomyłka. Dziękuję bardzo, dziękuję, panie pośle. Dziękuję.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę posłów sekretarzy o obliczenie wyników głosowania i przekazanie protokołu

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, zechce podnieść rękę.

Kto się wstrzymał? Proszę posłów sekretarzy o obliczenie wyników głosowania i przekazanie protokołu zbiorczego.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druków nr 286 i 286-A, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał? Proszę posłów sekretarzy o obliczenie wyników głosowania i przekazanie protokołu zbiorczego.

Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, tj.

Dziękuję bardzo.